Wysoka Izbo! Niestety znowu jest tak samo, tzn. znowu wczoraj o godz. 18 wpłynął projekt ustawy, który liczy 45 stron. Składam wniosek formalny o odroczenie obrad przynajmniej do jutra, żebyśmy mogli w spokoju nad tą ustawą popracować.

Już kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z aferą, kiedy państwo wzywali lekarzy, którzy od wielu lat nie żyją. Czy my naprawdę nie możemy w spokoju porozmawiać o ustawie? Czy naprawdę w spokoju nie możemy popracować nad ustawą i mieć na to więcej niż kilkanaście godzin? Panie marszałku, tak z ręką na sercu, czy pan tę ustawę przeczytał, te 45 stron, te ciężkie i wielkie zmiany, które dotyczą tego, jak będą traktowani lekarze w naszym kraju? Czy pan tę ustawę przeczytał w ciągu tej nocy? Czy to jest naprawdę dobry sposób na procedowanie? Panie pośle, ja byłem w lepszej sytuacji, bo znałem zarys tej ustawy już w zeszłym tygodniu.

Pan poseł Robert Winnicki z koła Konfederacji z wnioskiem formalnym. Wysoka Izbo! Kilka dni temu były marszałek sejmu litewskiego, pan Valinskas, powiedział o liderze Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, że takich ludzi należałoby rozstrzeliwać. A co więcej, od kilku tygodni trwa nagonka, która m.in. wpłynęła na wynik wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, nagonka prowadzona bezprawnie, nawet z punktu widzenia prawa litewskiego, na mniejszość polską na Litwie. Ta sytuacja łączy się z faktem, że od 2011 r. na Litwie obowiązuje skrajnie antypolska ustawa litwinizująca polskie szkolnictwo w tym kraju. W związku również z faktem, że cały czas jest problem z pisownią nazwisk, zwrotem majątków. Domagam się tego, żeby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wysłuchał sprawozdania ministra spraw zagranicznych w tym zakresie. Jak pan poseł dobrze wie, nie jest to wniosek formalny, ale nie przerywałem panu ze względu na znaczenie sprawy. Bardzo proszę. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 na podstawie art. 184 ust. 3 składam wniosek o przerwę w obradach Sejmu. Przerwę, która posłuży na wystosowanie zaproszenia na to posiedzenie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta, który niedawno uzyskał niezwykle silny mandat społeczny po wyborach. Przed wyborami uczestniczył w każdym istotnym działaniu związanym ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. Współuczestniczył w tworzeniu poszczególnych tarcz, proponował projekt dotyczący bonu turystycznego, kilka razy w tygodniu uczestniczył w konferencjach wspólnie z byłym ministrem zdrowia. A teraz co? Nawet wczoraj, kiedy powoływał ministra edukacji, [[Dzwonek]] nie zabrał głosu w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewicy, z wnioskiem formalnym. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i ponowny Konwent Seniorów, na którym dokonalibyśmy zmiany decyzji dotyczącej wyboru rzecznika praw obywatelskich. 2 miesiące - tyle Wysoka Izba zwleka z możliwością wyboru rzecznika praw obywatelskich. Nie dlatego, że nie było czasu, ale dlatego, że nie było chęci. Jedna kandydatka, tysiąc organizacji, które ją poparły, możliwość wyboru osoby, która ma wszelkie kompetencje do tego, żeby zasiąść w fotelu rzecznika praw obywatelskich. Ale do tego trzeba dobrej woli.

Rzecznik praw obywatelskich powinien mieć prawo głosu w tej Izbie, a skoro mamy jedyną kandydatkę, to to jest prawo, którego nie powinniśmy odmawiać sobie i Polsce. Dziękuję bardzo. Jak pan dobrze wie, jest to niezgodne z regulaminem. Mamy trzy wnioski o przerwanie obrad lub ich odroczenie.

Kto się wstrzymał?

Wniosek o przerwę został przyjęty.

Wysoki Sejmie! Przegłosowaliśmy wniosek o przerwę, ale także równocześnie o odroczenie obrad. Opozycja, ściślej mówiąc: Platforma Obywatelska, chce zablokować przyjęcie ustawy, na którą czekają Polacy. Ale głosowanie wypadło tak, jak wypadło. Zwołam wobec tego Konwent Seniorów i zwrócę się z propozycją do Platformy o wycofanie tego wniosku. Natomiast jeżeli wniosek nie zostanie wycofany, to będziemy zmuszeni przerwać obrady Sejmu do jutra.

Myślę, że to jest rozwiązanie rozsądne. Oczywiście jeżeli zwycięży totalna opozycja, tzn. totalny pomysł na przerwanie obrad Sejmu, to tak się stanie. Bardzo proszę, ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę Konwent Seniorów do saloniku.

Wznawiam obrady. Wysoki Sejmie!

Nie, to na wniosek Platformy Obywatelskiej. Tak jest, na wniosek. Pan nie ma teraz głosu, panie pośle Nitras. Ostrzegam pana. A więc na wniosek Platformy Sejm większością głosów uznał, że obrady odłożymy do jutra.

Platforma nie zgodziła się na to. Mam nadzieję, że nie. W tej sytuacji, skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra do godz. 9.